Dziękuję. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 1. porządku dziennego: Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie uczczenia 50. rocznicy Grudnia ’70 (druk nr 832) Bardzo proszę państwa posłów o powstanie. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uczczenia 50. rocznicy Grudnia ’70. 50 lat temu na Wybrzeżu doszło do jednych z najkrwawszych wydarzeń we współczesnych dziejach Polski. Bezpośrednią przyczyną protestów społecznych była podwyżka cen żywności ogłoszona przed zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia. 14 grudnia rozpoczął się strajk w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, a następnie w innych zakładach pracy w Gdańsku. Do protestu dołączyli pracownicy Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, Stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie, Zamechu w Elblągu i wielu innych zakładów na Wybrzeżu. Protestowano również w kilku innych miastach, m.in. w Białymstoku, Krakowie czy Wałbrzychu. Sprzeciw wobec podwyżki cen i wobec komunistycznej władzy przybrał formę strajków okupacyjnych, wieców i demonstracji ulicznych pod siedzibami komitetów partii. Protestujący i strajkujący domagali się wycofania podwyżki cen, podniesienia wynagrodzeń, poprawy warunków pracy i zwolnienia aresztowanych kolegów. Zamiast rozmowy i poszukiwania porozumienia władze PRL zdecydowały się na rozwiązanie siłowe, wysyłając na ulice miast oddziały wojska oraz milicji. Według oficjalnych danych podczas wydarzeń Grudnia ’70 śmierć poniosło 45 osób, ponad 1100 zostało rannych, a ponad 3 tys. aresztowano. Wiele osób straciło pracę. W pamięci Polaków szczególnie utkwił gdyński „Czarny czwartek”, gdy otworzono ogień do stoczniowców idących rankiem do pracy. Tragicznym symbolem tego dnia, ale i całego Grudnia ’70 stał się pochód idący za niesionym na drzwiach ciałem zabitego 18-letniego Zbigniewa Godlewskiego, znanego w grudniowym przekazie jako Janek Wiśniewski. Pamięć tragicznych wydarzeń Grudnia ’70 i dążenie do upamiętnienia jego ofiar stały się ważnym elementem tożsamości mieszkańców Wybrzeża, a w Gdańsku przyczyniły się do narodzin opozycji demokratycznej, czyli Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża i Ruchu Młodej Polski. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 50. rocznicę wydarzeń grudniowych składa hołd tym wszystkim, którzy protestując i sprzeciwiając się tzw. władzy ludowej, złożyli w ofierze swoje życie, narazili swoje zdrowie oraz karierę zawodową na uszczerbek, a także tym, którzy przechowali i przekazywali pamięć o Grudniu ’70. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża przekonanie, że Grudzień ’70 był jednym z etapów polskiej drogi wiodącej do Sierpnia ’80 i odzyskania przez Polskę niepodległości i wolności w 1989 r. Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały przez aklamację.

Bardzo państwu posłom dziękuję. Bardzo dziękuję. Mamy wnioski formalne. Bardzo proszę, pani poseł. Wysoki Sejmie! Sejm nie może być ani niemy, ani ślepy i głuchy na rzeczy, które dzieją się w Polsce. Wiemy, że wicepremier do spraw bezpieczeństwa zajmuje się bezpieczeństwem jednej jedynej osoby w kraju, swoim własnym. 13 grudnia ponad 80 radiowozów chroni jego mieszkania, kiedy kilka dni wcześniej policja łamie trzykrotnie rękę 19-letniej dziewczynie, prześladuje młodych protestujących. Domagamy się przerwy, zwołania Konwentu Seniorów i wprowadzenia pod obrady natychmiastowej pilnej informacji wicepremiera do spraw bezpieczeństwa na temat kosztów i sensowności działań Policji w ostatnich miesiącach przeciwko protestom kobiet, obywatelek i obywateli o wolność, demokrację i prawa człowieka. Oczywiście nie zwołam Konwentu Seniorów. Przegłosujemy ten wniosek. Poddam ten wniosek pod głosowanie.

Kto z pań i panów posłów jest za zarządzeniem przerwy w obradach, zechce nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Jeszcze jeden wniosek formalny, pan poseł Stefan Krajewski, Koalicja Polska. Bardzo proszę. Panie pośle, chciałam zapytać, czy to będzie wniosek o przerwę. To ciekawa jestem o co. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Na podstawie art. 184 wnioskuję w tym momencie nie o przerwę, ale o odroczenie posiedzenia do godz. 15 [[Wesołość na sali]] w celu zwołania Konwentu Seniorów i w celu uzupełnienia porządku obrad o informację prezesa Rady Ministrów o kryteriach przyznawania wsparcia dla samorządów z funduszu inwestycji lokalnych. Ponad 4 mld zł zostały podzielone w taki sposób, że samorządowcy do dziś są zbulwersowani. Do tego, że tutaj wszystko odbywa się bez żadnego trybu, już zdążyliśmy się przyzwyczaić, ale samorządowcy czekają na to, że będą mieli informację o tym, w oparciu o jakie kryteria zostały podzielone te środki, czy w oparciu tylko o przynależność do Prawa i Sprawiedliwości, czy w oparciu o realne potrzeby mieszkańców.

W związku z tym nie mam. Ale zgłosił pan wniosek o odroczenie. Proszę bardzo, proszę bardzo. Złożony został wniosek formalny o odroczenie posiedzenia. Poddam ten wniosek pod głosowanie. Kto z pań i panów posłów jest za odroczeniem posiedzenia, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 2. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 (druki nr 640 i 785) Proszę pana posła Henryka Kowalczyka o przedstawienie sprawozdania komisji.

Wysoka Izbo!

Pierwsze czytanie tego projektu odbyło się w dniu 7 października, po czym projekt został skierowany do Komisji Finansów Publicznych celem przedstawienia sprawozdania do 2 grudnia. Komisja Finansów Publicznych rozpatrzyła projekt zgodnie z przyjętym przez Prezydium Sejmu harmonogramem prac, a efektem tychże prac jest sprawozdanie prezentowane w druku nr 785.

Komisja Finansów Publicznych na swoich posiedzeniach rozpatrywała własne części budżetowe, ponadto rozpatrywała opinie innych komisji sejmowych w zakresie określonym postanowieniem marszałka Sejmu.

W trakcie posiedzeń komisji posłowie przedstawiali najważniejsze informacje z dyskusji na posiedzeniach innych komisji, a także zadawali szereg szczegółowych pytań dotyczących m.in. zaplanowanych budżetów niektórych jednostek cieszących się dużą autonomią budżetową, takich jak Kancelaria Prezydenta, kancelarie Sejmu i Senatu, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich czy Najwyższa Izba Kontroli. Szczególne zainteresowanie posłów budziły m.in. kwestie dotyczące założeń makroekonomicznych budżetu, deficytu, długu publicznego czy skuteczności administracji podatkowej, kwestie dotyczące zatrudniania i poziomu wynagrodzeń w poszczególnych jednostkach administracyjnych, także finansowania uczelni wyższych, kultury, opieki społecznej, opieki nad zabytkami.

Były to opinie pozytywne, jedynie Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki przedstawiła dwie poprawki, a Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka dołączyła dwa zdania odrębne.

Siedem poprawek dotyczyło załączników.

Tak jak powiedziałem, zgłoszonych zostało 715 poprawek. Ponad 200 poprawek wskazywało jako źródło finansowania część: Obrona narodowa.

Kolejnym takim źródłem finansowania poprawek był Instytut Pamięci Narodowej, ponad 100 poprawek na łączną kwotę ponad 3 mld zł.

Źródło finansowania: IPN, a tam jest tylko 412 mln. Podobnie CBA.

Fundusz Kościelny, ulubieniec Lewicy.

Myślę, że warto zauważyć, że sam poseł Krzysztof Paszyk złożył ponad 100 poprawek o mniejszej skali, ale za to doceniając prawie każdą gminę w swoim okręgu.

Dziękuję, panie pośle. Myślę, panie pośle, bo pozwolę sobie tak jednym zdaniem skomentować to, co pan powiedział w sprawie łączenia tych kwot, że może to jest tak, że opozycja po raz pierwszy nie zaufała, że po prostu.

Proszę państwa, witam państwa. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 15-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 5-minutowego oświadczenia w imieniu koła. Serdecznie zapraszam pana posła Henryka Kowalczyka z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, aby przedstawił stanowisko tego klubu w sprawie budżetu. Zapraszam pana posła. Panie Marszałku! Ja oczywiście nie śmiałem się z poprawek, tylko przedstawiałem fakty, jak te poprawki zostały złożone. Projekt został przygotowany z uwzględnieniem trudnej sytuacji makroekonomicznej wynikłej z pandemii COVID-19, która rozprzestrzeniła się błyskawicznie na całym świecie i przyczyniła się do wywołania kryzysów gospodarczych na niespotykaną dotychczas skalę.

Tak naprawdę będzie to powrót do poziomu z 2019 r.

To, że obecny, co warto zauważyć, zakładany spadek jest w przewidywaniach teraz już pewnie mniejszy, to jest ogromna zasługa rządu, który skutecznie pomagał przedsiębiorcom, co szczególnie było to widać w okresie wiosennej pandemii, bardzo skutecznie chroniąc miejsca pracy. Trudno przewidzieć rozwój pandemii, czy będzie jeszcze trzecia fala, czy pandemia już wygaśnie.

Należy uznać, że polskie finanse publiczne w tej niezwykle trudnej sytuacji wywołanej pandemią są bardzo bezpieczne. Reasumując, warto podkreślić, że projekt budżetu na 2021 r. opracowano przy zapewnieniu środków finansowych niezbędnych do kontynuacji dotychczasowych priorytetów rządu w zakresie zadań polityki społeczno-gospodarczej, w tym szczególnie aktywnej i ambitnej polityki społecznej. Choćby w zakresie 500+ żadnych planów redukcji tego typu wsparcia się nie przewiduje.

Dziękuję bardzo.

Proszę, panie pośle. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chcę omówić dwa bardzo istotne aspekty budżetu: bezpieczeństwa państwa i inwestycji, a przede wszystkim sprawy wewnętrzne, w tym kwestie służb mundurowych, obrony narodowej.

W tym główne wydatki obejmują emerytury i renty, wynagrodzenia i wydatki bieżące - 11,1 mld zł, wydatki majątkowe - 385 mln zł, przede wszystkim wydatki na takie formacje, jak: Centralne Biuro Śledcze Policji, Komenda Główna Policji, Straż Graniczna, Służba Ochrony Państwa, Komenda Główna PSP. Dodatkowo bardzo ważne fundusze, które uzupełniają funkcjonowanie tej sfery, stanowią Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, Fundusz Wsparcia Policji, Fundusz Wsparcia Straży Granicznej oraz Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

na inwestycje samorządowe, powiatowe i gminne. Ten tak oczekiwany i świetnie zresztą realizowany program przez samorządowców we współpracy z wojewodami w roku przyszłym również będzie kontynuowany.

Program idzie doskonale, można powiedzieć: znakomicie, nabiera tempa, i sądzimy, że rok 2021 będzie następnym rokiem bardzo dużych inwestycji zauważanych na polskich kolejach. Punkt następny dotyczy programu specyficznego, ale bardzo istotnego „Mosty dla regionów”

To bardzo istotna, ogromna inwestycja, która zmieni ten zakres, który w tej części Polski jest bardzo istotny. Proszę państwa, reasumując, inwestycje, inwestycje, inwestycje i bezpieczeństwo - to jest ogromny element naszego budżetu. Dziękuję serdecznie. Jest. Proszę bardzo. Wysoka Izbo! Jednym z ważniejszych zadań budżetowych państwa jest finansowanie ochrony zdrowia Polaków. Ten imperatyw jest szczególnie ważny w czasie pandemii.

Zaplanowano w tej kwocie dofinansowanie programów polityki zdrowotnej - wzrost o 357 mln zł.

Jest to wzrost o 202% w stosunku do 2020 r.

Ważnym działem budżetu państwa jest dział 855: Rodzina. Obejmuje on pomoc państwa w wychowaniu dzieci, świadczenia rodzinne, pomoc osobom uprawnionym do alimentów, wypłacanie zasiłków dla opiekunów, program „Za życiem”, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, opiekę nad dzieckiem do 3. roku życia, Kartę Dużej Rodziny, rządowy program „Dobry start”, a przede wszystkim świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”, na który zaplanowano w 2021 r. 41 mld zł.

Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano w budżecie blisko 12,9 mld zł, tj. ponad 551 mln więcej aniżeli w bieżącym roku.

Będzie to waloryzacja procentowo-kwotowa z gwarantowanym dodatkiem 500 zł. Planowane są również dla emerytów i rencistów trzynasta i czternasta emerytura. Świadczenia te będą wypłacane z Funduszu Solidarnościowego w łącznej wysokości ponad 23 mld zł. Panie Marszałku! Ważną częścią budżetu państwa dla samorządów jest subwencja ogólna.

Największą częścią tej subwencji jest część oświatowa, która wynosi ponad 52 mld zł i jest większa o 2200 mln zł aniżeli w roku 2020. Pozostałe subwencje wynoszą łącznie 18 mld zł, a ich wzrost wynosi ponad 7%. Chcę zaznaczyć, że ministerstwo zmieniło algorytm rozdziału subwencji o światowej.

To oznacza, że subwencja na ucznia w takiej szkole wzrośnie z 611 zł do 917 zł. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę pana posła Cezarego Tomczyka, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Zapraszam, panie pośle. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jak do finansów państwa podchodzi ten rząd, widać po dzisiejszej debacie, i to nie tylko dlatego, że po stronie PiS-u właściwie nie ma żadnych posłów, oprócz posłów, którzy zabierali głos, ale także dlatego, że nie ma też z nami ministra finansów.

Zawsze minister finansów to był ktoś. To był ktoś, kto dbał o interesy państwa. Dzisiaj to jest ktoś, kto dba tylko o interesy PiS-u. Zwracam się bezpośrednio z tego miejsca do Polek i Polaków śledzących tę debatę w swoich domach, bo właśnie ta debata o budżecie jest jedną z tych najważniejszych. Od stanu państwa zależy dziś los każdej polskiej firmy, od stanu finansów państwa zależy dziś los każdego pracownika. Chcieliśmy zaprezentować dziś właśnie stan polskiego państwa w trzech aktach i niestety jest to dramat. Akt pierwszy: umierają ludzie. Ten rząd przyczynił się do śmierci kilkudziesięciu tysięcy Polek i Polaków. Tylko w listopadzie zmarło 30 tys. osób więcej niż w listopadzie ub.r. Tylko 10 tys. osób zmarło na COVID, 20 tys. to zgony, których można było uniknąć. To jest skutek nieprzygotowania służby zdrowia na epidemię, to jest skutek braku sprzętu, maseczek, tlenu, przyłbic, respiratorów. W listopadzie, porównując rok do roku, zmarło w Polsce najwięcej ludzi od II wojny światowej. Akt drugi: umierają firmy. Fatalne zarządzanie epidemią, chaotyczne decyzje prowadzą do upadku firm, restauracji, barów, kin, teatrów, siłowni, jednoosobowych działalności gospodarczych. Ten rząd zlekceważył epidemię. Już teraz gospodarkę można byłoby otwierać, tak jak robi się to na południu Europy, kiedy po świętach gospodarka wraca do normalności, bo rząd nie lekceważył epidemii. Prawda jest taka, że dopóki ten rząd przegrywa z epidemią, dopóty z tym rządem przegrywać będą polskie firmy. I trzeba to powiedzieć jasno, że te przedłużające się obostrzenia to jest wina tego rządu, który po prostu nie radzi sobie z epidemią. I wreszcie akt trzeci: umiera gospodarka. To jest kluczowy akt i właśnie o tym jest ta debata, debata budżetowa na rok 2021. Polski rząd po raz kolejny robi coś zupełnie innego niż większość krajów Unii Europejskiej. Podczas gdy cała Europa oszczędzała na trudne chwile, takie jak ta, i teraz pomaga swoim firmom, lokując tysiące euro w tych firmach, w Polsce trwał bal PiS. Dla Rydzyka 250 mln zł, na Telewizję Polską, szczujnię propagandową, 2 mld zł, samoloty dla władzy, proszę bardzo, 2 mld zł bez przetargu. Tysiąc limuzyn zamiast karetek - kto bogatemu zabroni. Najdroższy szpital na świecie bez pacjentów na Stadionie Narodowym, 2 km stąd, każdy może przekonać się na własne oczy. I teraz jest dokładnie tak samo, pod osłoną epidemii ten rząd wprowadza nowe podatki dla Polek i Polaków, a dokładnie będzie to 10 nowych podatków. Poproszę o pierwszy slajd. To jest odpowiedź rządu na to, że polskie firmy dzisiaj umierają. Ludzie protestują w całej Polsce, bo po prostu mają rację. Zażynacie polskie firmy, zażynacie polską gospodarkę i wolność też zażynacie. Premier Morawiecki mówił, że jesteśmy liderami w Europie. Liderami w podnoszeniu podatków - to na pewno. Nie dość, że wprowadzacie 10 podatków, to jeszcze podwyższacie podatki, które istnieją. Zmieniacie ich stawki po to, żeby Polacy do budżetu państwa musieli wpłacać więcej, w takim momencie, kiedy pieniądze są potrzebne. Spójrzmy: Belgia. Zobaczmy, jak to jest w Europie. Belgia. Belgia obniża VAT na katering, żywność i napoje bezalkoholowe do 6%. Co robi w tym czasie polski rząd? Oto polski rząd wprowadza podatek cukrowy, żeby żywność była droższa, jeszcze droższa. Austria. Austria obniża VAT z 10% do 5% dla sektora gastronomicznego, kulturalnego i wydawniczego. Jaka jest odpowiedź polskiego rządu? Podwyższenie abonamentu radiowo-telewizyjnego na tę PiS-owską szczujnię. Irlandia. Polski rząd utrzymuje podwyższony VAT, który miał obniżyć lata temu. Bułgaria obniża VAT w restauracjach i w przemyśle rozrywkowym. Co robi polski rząd? Polski rząd wprowadza podatek handlowy. Niemcy. Niemcy obniżają główną stawkę VAT z 19% do 16%. Polski rząd co robi? Podwyższa składki na ZUS. To jest odpowiedź dla Polaków i dla polskich firm. Czechy. Czechy obniżają podatek PIT z 20% do 15%. Co robi polski rząd? Polski rząd wprowadza podatki za deszcz. I na koniec ostatnia sprawa, kwestia cen. Poproszę ostatni slajd. W ciągu 5 lat rząd PiS wprowadził ok. 35 nowych podatków i opłat, teraz kolejne 10. Ale to nie wszystko, bo oprócz tego, że z kieszeni polskich obywateli polski rząd chce wyciągnąć dodatkowe miliardy złotych i niszczyć polskich przedsiębiorców, dzisiaj mamy w Polsce galopujące ceny. To jest wykres, który pokazuje, że inflacja w październiku była najwyższa w Europie, najwyższa w Unii Europejskiej. Co to jest inflacja? To jest po prostu fakt, że pieniądz ma mniejszą wartość, a ceny rosną. Ceny w Polsce rosną średnio 13 razy szybciej niż w Unii Europejskiej. Jaki jest drugi kraj w Europie, jeśli chodzi o inflację, drugi w kolejności? Węgry. Rzeczywiście mamy z kogo brać przykład. I to niestety jest nasz dramat, za który odpowiada premier Morawiecki i ten rząd. Dziękuję bardzo. Pani poseł Izabela Leszczyna, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Cudze pieniądze to poważna sprawa, dlatego gdy rozmawiamy o budżecie państwa, czyli o pieniądzach podatników, trzeba sobie postawić kluczowe pytanie, dlaczego właściwie rząd zabiera ludziom pieniądze? Odpowiedź wydaje się prosta. Po to, żeby zapewnić obywatelom dobrą ochronę zdrowia, dobrą edukację, bezpieczeństwo, czyli po to, żeby życie ludzi było lepsze, żeby byli zdrowsi, żeby żyli dłużej, byli lepiej wykształceni, czuli się bezpiecznie na ulicach polskich miast, po to, żeby nasza ojczyzna była bezpieczna i miała wokół więcej przyjaciół niż wrogów. Żeby pokazać, czy rząd osiąga swoje cele, wymyślono różne wskaźniki.

A pan mówi, że to bezpieczne.

Ale co się stało w roku 2019? Rozszczelniło się. Proszę wrócić do tego slajdu.

Tutaj panowie posłowie chwalili się: będzie 500+, będzie trzynasta, czternasta emerytura, a premier Morawiecki mówił, że cała piątka Kaczyńskiego będzie sfinansowana z redukcji luki VAT. Proszę o kolejny slajd. Tak to wygląda, moi kochani.

A ile potrzebujecie na 500+ oraz trzynastą i czternastą emeryturę? To skąd weźmiecie 50 mld zł? Ten slajd czarno na białym pokazuje to, że rachunek za obietnice PiS muszą zapłacić Polacy. Co jeszcze rośnie w państwie rządzonym przez PiS? Kolejki do lekarzy. Ale nie pokażę wam statystyk, bo rząd PiS kazał je ukryć. W dodatku ludzie umierają zanim doczekają się swojej wizyty.

Czy w związku z tym w budżecie na 2021 r. mamy więcej pieniędzy? Nie. Przyznał to z wielką szczerością i dumą pan poseł Szlachta. Jak panu nie wstyd? Przecież mamy pandemię, a PiS idzie wstydliwą ścieżką dojścia do 6% PKB w 2024 r. Zachowujecie się tak, jakby system ochrony zdrowia nie był na skraju wydolności, jakby nic się nie stało, jakby nie było pandemii. Minister zdrowia opowiada jakieś banialuki, recovery plan zapowiada. Z czego? W budżecie nie dali na to ani złotówki. Klub Koalicji Obywatelskiej z tego waszego budżetu przesuwa 7 mld zł na ochronę zdrowia, bo chcemy ratować życie Polek i Polaków, bo przy was są po prostu zagrożeni. Powiedziałam, że to, co powinno rosnąć, spada. Na co rząd powinien przeznaczać podatki? Na to, żeby długość naszego życia rosła. Powinna też rosnąć liczba aktywnych zawodowo osób. To jest nasza przyszłość, to jest rozwój gospodarki. Powinna rosnąć wartość spółek Skarbu Państwa, a ona spada. Na szczęście spada też zaufanie do rządu.

Ile z tych osób to obywatele naszej ukochanej ojczyzny? 233 tys., tj. 80% wszystkich ludzi, którzy przestaną w przyszłym roku w Europie pracować, to są Polacy, a przecież Polacy to tylko 8% populacji Unii Europejskiej. Bardzo cieszę się z tego, że ci młodzi ludzie to rozumieją. Ci młodzi, którzy protestują od wielu tygodni na ulicach, robią to nie tylko w obronie polskich kobiet, oni pogonią was z ministerstw, w których siedzicie i myślicie tylko o tym, jak podnieść sobie płace, jak zatrudnić kolejnych kolegów albo co najwyżej jak przekopać Mierzeję Wiślaną. Oni pogonią was z ministerstw, bo są mądrzy, bo nie udał wam się plan marszałka Terleckiego, żeby kolejne pokolenia młodych wychować tak, żeby głosowali na PiS. Wszystko to, co tym młodym ludziom zrobili szkodnicy tacy jak Zalewska, Piontkowski czy Czarnek, obróci się przeciwko wam, zapłacicie za to, bo zasłużyliście. Teraz okazało się, że kawałek trzeba podjechać pod górę. Dla PiS-u to jest proste, oni wiedzą, skąd dosypać pieniędzy. Zresztą prezes banku Mateusz Morawiecki już wiele lat temu przedstawił swoją koncepcję rozwoju gospodarki. Powiedział przecież wszystkim wprost, że ludzie mają pracować za miskę ryżu. Podsumowując, zapytam: Czy zabierając Polkom i Polakom tak dużo pieniędzy z podatków, składek, danin i różnych opłat, rząd PiS-u przez te 5 lat sprawił, że Polacy są zdrowsi? Nie. Czy Polacy żyją dłużej? Nie. No to może czują się bezpiecznie na ulicach polskich miast? Też nie, mówiła o tym pani poseł Barbara Nowacka. No to może mamy chociaż więcej przyjaciół na świecie? No niestety, też nie. To znaczy, że rząd PiS-u stracił moralne prawo do rządzenia Polską, i większość społeczeństwa o tym wie. Nie wie jeszcze tylko rząd PiS-u, ale niebawem zrozumie, że każdy kolejny dzień rządu PiS to dramat dla Polski i że będziemy musieli odrabiać to przez wiele, wiele lat. Dziękuję serdecznie. Zapraszam pan posła Dariusza Wieczorka, klub parlamentarny Lewica. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Wiem, że jest zastępca, ale myślę, że szacunek dla tej Izby wymaga, żeby dzisiaj w trakcie tej najważniejszej debaty jednak pan minister był. Rozumiem, że nie ma pana premiera, bo walczy z panem ministrem Ziobrą, więc może nie mieć czasu zajmować się sprawami budżetowymi, [[Oklaski]] ale pan minister powinien jednak z nami być. Usłyszeliśmy tutaj od pana przewodniczącego Kowalczyka i przedstawicieli PiS-u, że w tym budżecie najważniejsza sprawa to inwestycje, inwestycje i bezpieczeństwo. Mam pytanie: Czy panowie rzeczywiście czytaliście druk nr 640? Bo mam wrażenie, że czytaliście jakiś inny druk. To czas kryzysu, a wiadomo, że w czasie kryzysu potrzeba mądrych decyzji, mądrej władzy. Potrzeba decyzji, które będą, mówiąc krótko, z tym kryzysem walczyły. Niestety ten projekt budżetu pokazuje, że to jest tylko i wyłącznie emanacja obecnej władzy Prawa i Sprawiedliwości.

To budżet chaosu, stagnacji i braku wizji państwa po pandemii. A więc rodzi się pytanie: Czy to jest deficyt realny, czy czasami znowu nie ukrywacie jakichś rzeczywistych wydatków? Bo mamy w tym zakresie już bardzo poważne doświadczenia.

Wybory są za trzy lata. Uczciwie dzisiaj mówmy o tym, że rzeczywiście mamy z tym problem, bo dzisiaj lepsza jest najgorsza prawda niż takie kombinowanie i ukrywanie, i mówienie sobie z tej mównicy m.in., że wszystko jest w porządku i wszystko jest ok. Według polskiej metody liczenia długu publicznego oczywiście mamy te 51%, 52%, ale jak już zastosujemy unijne metody liczenia długu publicznego, to w tym budżecie, który planujecie, on będzie wynosił już prawie 65%. W tym kontekście oczywiście, mimo tych wszystkich sporów i tych gorących dyskusji tutaj, na tej sali, dobrze się stało, że Polska nie zawetowała budżetu Unii Europejskiej, nie zawetowała Funduszu Odbudowy, bo prawda jest taka, że mielibyśmy w ogóle problem z konstrukcją budżetu na rok 2021. Pewnie ten budżet trzeba będzie ze względu na te środki unijne oczywiście nowelizować, ale to będzie bardzo poważny wkład w ten budżet i w ratowanie polskiej gospodarki.

Tutaj z tej mównicy często pan premier mówił, że opozycja nie ma pomysłu na to, jak działać, jak funkcjonować.

Oczywiście bardzo byśmy wszyscy chcieli, żeby tak rzeczywiście było, ale pytanie: Czy tak będzie i czy czasami nie mamy tutaj do czynienia z zbyt wielkim optymizmem?

Jakie czynniki mają spowodować, że inflacja w tym roku będzie spadać? Po spadku inwestycji w 2020 r. o 10% planujecie, że nastąpi ich wzrost o 4%, ale prawda jest taka, że ten wzrost inwestycji nastąpi tylko i wyłącznie dzięki temu, że będą to inwestycje wojskowe, bo realnie udział środków inwestycyjnych w tym budżecie to jest ok. 7,3%. Kolejna ciekawa sprawa przy tych założeniach to kwestia dotycząca spadku spożycia, który miał miejsce w roku 2020, o 2,6%.

I teraz rodzi się pytanie: Jak to się dzieje, że nie planujecie wzrostu wynagrodzeń, nie dajecie wynagrodzeń dla lekarzy, zabieracie fundusze nagród w służbach mundurowych, nie zwiększacie pensji nauczycielom, nie zwiększacie pensji w budżetówce, wzrasta bezrobocie, a konsumpcja ma wzrosnąć? Przyznam się szczerze, że jest to bardzo ciekawe podejście, i myślę, że komuś należy się rzeczywiście Nobel z ekonomii za tego typu wyliczenia. Jaka jest konstrukcja tego budżetu? Otóż rzeczywiście ta konstrukcja powoduje, po pierwsze, zmniejszenie podatku CIT, ale wzrost wpływu z podatku VAT do 181 mld, wzrost wpływu z podatku PIT do 89 mld, spadek dochodów jednostek budżetowych. Logika takiego konstruowania obciążeń i przekazywania transferów nie jest widoczna dla przeciętnego Polaka i przeciętnego podatnika, który dostrzega tylko tę bieżącą pomoc pieniężną. Programy 500+, trzynasta emerytura i inne świadczenia - wszystko to bardzo ładnie wygląda w tej propagandzie, mówimy o tym, że pomagamy, że wszystko jest okej. Ale jak Polacy zobaczą rachunki za energię elektryczną, zobaczą rachunki za prąd, zobaczą rachunki za paliwo, zobaczą rachunki w sklepach, to nagle się okaże, że to, co dajecie, po prostu zabieracie. Rząd PiS-u daje i zabiera. A wiecie państwo, co się dzieje, jak ktoś daje i odbiera? To się w piekle poniewiera. Przestrzegamy przed tym, bo taka jest właśnie wasza filozofia. Brak było oczywiście uczciwej debaty dotyczącej tego, jakie pomysły można realizować w tym trudnym 2021 r., bo zwracaliśmy uwagę w trakcie posiedzeń komisji i debaty sejmowej, że to będzie naprawdę inny rok. To będzie rok po pandemii i nie można tego tak traktować, że tutaj nic się nie stało, że to jest ten sam budżet. Lewica zaproponowała stworzenie Funduszu Odbudowy Gospodarki. To jest nasz pomysł na wyjście z tego kryzysu. Fundusz Odbudowy Gospodarki jako fundusz celowy, fundusz, który miałby za zadanie być szybką reakcję na to, co się dzieje, oparty byłby oczywiście na trzech głównych filarach, tj. zdrowiu, przedsiębiorczości i samorządności. To jest propozycja bardzo konkretna, nad którą chcieliśmy wspólnie pracować. To propozycja, która ma na celu jedną rzecz, a mianowicie, po pierwsze, zasilenie tego funduszu poprzez przesunięcia w budżecie, w projekcie budżetu na rok 2021, kwotą 20 mld zł. I zwracamy uwagę na główne pozycje, które by ten fundusz tworzyły. To przede wszystkim zmniejszenie do 2% PKB nakładów na wojsko i obronę narodową. Jeszcze raz z uporem godnym tej sprawy będziemy mówić: dzisiaj do walki z koronawirusem i walki o miejsca pracy nie potrzeba nam czołgów, armat, samolotów, pistoletów. Dzisiaj potrzeba armii ludzi, armii lekarzy, gigantycznych środków, żeby przede wszystkim pomóc przedsiębiorcom. W tym kontekście, jak mówimy o ochronie zdrowia, jest w budżecie rezerwa celowa blisko 5 mld zł. Nie ma co trzymać tych środków w rezerwie celowej, trzeba je po prostu już dzisiaj uruchomić. Dodatkowo są kwestie dotyczące dywidend, dodatkowo są kwestie dotyczące likwidacji niektórych funduszy, które stworzyliście w tym funduszu prywatyzacji spółek, bo widzimy, że aktywna jest dzisiaj polityka i zaczynamy już to wszystko rozumieć, po co te fundusze powstają, po co tam chcecie zgromadzić 1,5 mld zł. Pan przewodniczący Kowalczyk mówił o tym Funduszu Kościelnym, o IPN-ie. To jest 20 pozycji, z których te 20 mld zł można rzeczywiście przesunąć i można te środki wydać właśnie na tworzenie tego funduszu. Dodatkowo w tym funduszu - i to jeszcze raz chcę podkreślić - dzięki tej decyzji, że nie ma weta, znajdzie się przez najbliższe 3 lata kwota 103 mld zł z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej. I oczywiście to jest kwota, która w trakcie roku po pozytywnych decyzjach Parlamentu może zasilić ten fundusz w wysokości ok. 42 mld zł, bo jeżeli sobie rozłożymy te kwoty na 3 lata, to propozycja nasza jest taka, żeby przez pierwsze 2 lata to była kwota zasilająca ten fundusz 42 mld zł, a w ostatnim roku, w roku 2023, żeby to była kwota 19 mld zł.

I jaka jest koncepcja, którą tutaj polskiemu rządowi przedstawiamy? Otóż, jeżeli mówimy o filarze: zdrowie, to mówimy o tym, że jest potrzebny restart w ochronie zdrowia. Dzisiaj wiemy, że szpitale powiatowe, wojewódzkie, państwowe borykają się z wielkimi problemami finansowymi. Trzeba doposażyć te szpitale po pandemii, trzeba dzisiaj znaleźć środki na to, ażeby te szpitale mogły zacząć normalnie funkcjonować, a więc taki restart inwestycji w szpitalach w wysokości 16 mld zł jest absolutnie potrzebny. Tego nie ma co się bać. Wy nie chcecie dawać podwyżek lekarzom, nie chcecie dbać o ochronę zdrowia, a dzisiaj, w okresie pandemii, jest to absolutnie kluczowa sprawa. Tu musimy zdać sobie sprawę z jednej rzeczy, że mianowicie dzisiaj te małe i średnie przedsiębiorstwa to jest klucz do tego, żeby polska gospodarka normalnie mogła funkcjonować. Uważamy, że na restart - podkreślam: restart - tych małych i średnich przedsiębiorstw trzeba przeznaczyć ok. 10 mld zł.

W związku z tym to są środki, które są niezbędne, żeby nasze firmy mogły normalnie funkcjonować. I wreszcie filar: samorządność - 18 mld zł - filar inwestycje samorządowe i restart inwestycji samorządowych. Trzeba uczciwie powiedzieć: jeżeli samorządy mają dzisiaj inwestycje własne, to dajemy wam 50%, dopłacamy do tych inwestycji 50%, co zwolni wam środki w budżetach na inne cele i na normalne funkcjonowanie. I do tego oczywiście nowoczesna edukacja. Tu nie ma co się tego obawiać, to po prostu trzeba zrobić. Cel to jest ochrona miejsc pracy, 1 mln miejsc pracy i 100 tys. przedsiębiorców. Taki powinien być cel tego budżetu. Dlatego, jeżeli ten projekt budżetu nie będzie w taki sposób zmieniony, polska lewica nie będzie takiego budżetu popierać. Dziękuję serdecznie, panie pośle. Zapraszam pana posła Krzysztofa Paszyka, Klub Parlamentarny Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści. Bardzo proszę. Panie i Panowie Posłowie! Panowie Ministrowie! Przed chwilą z ust przedstawiciela Zjednoczonej Prawicy, przedstawiciela większości sejmowej zasiadającej na tej sali, usłyszeliśmy, że budżet państwa na 2021 r. to budżet inwestycji i budżet bezpieczeństwa. Coś się chyba państwu pomyliło, bo racjonalnie patrząc na ten budżet, niewiele on ma i z inwestycjami, i z bezpieczeństwem wspólnego. Jeśli chodzi o inwestycje, to ja dziękuję, jeśli inwestycje w Polsce mają wyglądać tak, jak Centralny Port Komunikacyjny, czyli narodowe betonowanie setek hektarów bez większego sensu, bez wyraźnego celu. No, chyba żeby się przypodobać panu prezesowi Kaczyńskiemu, ale to nie tak powinny być konstruowane i planowane w Polsce inwestycje, które pochłoną tyle środków. Teraz jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to niewiele ma z bezpieczeństwem wspólnego budżet państwa, który uporczywie ukrywa wszelki dług publiczny w naszym kraju. Niewiele wspólnego z bezpieczeństwem ma konsekwentne niedofinansowanie służby zdrowia. Przed rokiem, przed wyborami podpisaliście pakt dla zdrowia.

Ten cel już gdzieś umknął. Czy z bezpieczeństwem ma coś wspólnego zaprzestanie finansowania trzynastych emerytur?

Nie ma wyborów, nie ma trzynastej emerytury. Ale co mamy w budżecie i co jest bardzo nieładnym gestem wobec tych, którzy czekali na te trzynaste emerytury? Ano konsekwentne, hojne wspieranie telewizji Jacka Kurskiego. Bezpieczeństwo to również bezpieczeństwo żywnościowe. Mówi polskim rolnikom, że poziom finansowania będzie wynosił ok. 47 mld. To ja dzisiaj z tego miejsca przypomnę polskim rolnikom, że poziom finansowania ze środków krajowych naszego rolnictwa w roku 2016, czyli ostatnim roku, który był budżetowo układany przez Polskie Stronnictwo Ludowe, to było blisko 10 mld więcej. Tak wygląda wsparcie polskiego rolnictwa, zwłaszcza w dobie wielkiego kryzysu, który je dotyka, bo rolnicy to też przedsiębiorcy, to też są ludzie, których dzisiaj dotyka poważny kryzys.

Kwestia samorządów. To jest w szczególności rzecz niezwykle bulwersująca, gdy się obserwuje budżet państwa. Kolejne obciążenia są na barki samorządów nakładane, natomiast w ślad za tym nie idzie w ogóle finansowanie. A już szczytem tego, jak traktujecie samorządy, była - o tym dzisiaj mój kolega klubowy pan Stefan Krajewski mówił - kwestia podziału funduszu wsparcia. Pozwalam sobie w imieniu klubu Koalicja Polska złożyć ok. 200 poprawek, które zostały przygotowane przez samorządy w całym kraju.

Takie kryterium jest dzisiaj pokazane. To jest swoistego rodzaju szczucie samorządów, szczucie tych, którzy ostatnie lata swojej kariery poświęcili na zarządzanie sprawami lokalnymi - właśnie takie podejście.

Panie Marszałku! Kończąc swoje wystąpienie, chcę powiedzieć, że w tym kształcie budżet państwa nie daje możliwości, aby Koalicja Polska mogła go poprzeć. Te poprawki, które na pańskie ręce złożę, też są pewnego rodzaju wyrazem niezadowolenia z tej polityki realizowanej dzisiaj przez większość sejmową wobec lokalnych potrzeb. Dziękuję serdecznie, panie pośle. Bardzo proszę, pan poseł Dariusz Klimczak, Klub Parlamentarny Koalicja Polska. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Jeżeli chodzi o wysokość, to czy państwo zapomnieli już, jaką wysokość nakładów w stosunku do PKB państwo obiecali rezydentom? Czy oni od nowa mają protestować, podejmować protest głodowy, żebyście sobie przypomnieli, jakie obietnice rząd złożył? Przecież to jest nie fair, tak się, panowie, nie robi, szczególnie w stosunku do młodych ludzi, którzy są przyszłością naszego kraju, medyków, którzy są bohaterami naszych czasów. A biorąc pod uwagę to, że przekroczyliście ponad 2% na obronność, to znaczy, że źle definiujecie dzisiaj wroga w Polsce. Te priorytety są źle ustawione. To, o czym mówi Koalicja Polska - PSL, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści, to przede wszystkim zwiększenie nakładów na wynagrodzenia dla wszystkich medyków, bohaterów naszych czasów, bohaterów tej epidemii.

Ja to sprawdziłem i zapytałem laborantów z jednego ze szpitali w województwie łódzkim, jak sytuacja się ma. Dyrektor tamtejszego szpitala wystąpił o interpretację do ministerstwa i okazuje się, że nie należą się takie dodatki tym laborantom, mimo że pracują w szpitalu COVID-owym, ponieważ nie robią testów na COVID metodą PCR. Dlatego upominamy się, żeby wszyscy w szpitalach COVID-owych, lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, laboranci, opiekunowie medyczni, panie i panowie salowi, technicy, wszyscy ci, którzy są narażeni na zakażenie, dostawali tego typu premie.

Znowu zaniedbujecie kwestię specjalizacji. To powinien być absolutny priorytet w budżecie państwa. Dzisiaj jest absolutnie okazja do tego, żeby przekonać wszystkich tych, którzy chcą przeznaczyć pieniądze na inne działy, że tutaj jest niezwykle ważna sprawa. To samo dotyczy prywatnej ochrony zdrowia, o której my jako Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe mówimy, że trzeba zaangażować ten dział naszej gospodarki w leczenie pacjentów, przed którymi drzwi są zamknięte w publicznym systemie ochrony zdrowia. Zaczęliście to robić w stosunku do pacjentów COVID-owych, zróbmy to w stosunku do osób, które chorują na inne schorzenia. To samo dotyczy szczepionek. Dzisiaj musimy absolutnie walczyć z antyszczepionkowcami.

Przecież każdy rodzic wie, że taka szczepionka combo, stosowana, żeby nie szczepić dziecka kilka razy, jest naprawdę bardzo droga. Dzisiaj z takimi inicjatywami trzeba wyjść. Wiemy, że w tym budżecie braknie pieniędzy na ogłaszanie nowych konkursów dla NFZ-etu. A znamy przykłady z całego kraju, gdzie m.in. hospicja czekają na nowe kontrakty. Tak samo jest wiele zapytań o ogłoszenie nowych konkursów, np. szpital w Opocznie nie może od dłuższego czasu doprosić się o ogłoszenie konkursu na ginekologię i położnictwo. Bardzo proszę, żeby tego typu kwestie były poruszone w tym budżecie. Dziękuję, panie pośle. Bardzo proszę pana posła Jacka Protasiewicza, Klub Parlamentarny Koalicja Polska, a więc ten sam, który był poprzednio. Proszę bardzo. Panie Marszałku! W imieniu naszego klubu, ale też jako poseł ziemi dolnośląskiej, chociaż koledzy z okręgu kujawsko-pomorskiego również prosili mnie o złożenie dodatkowych poprawek, chciałbym złożyć poprawki, które dokładnie rekompensują samorządom gminnym, samorządom powiatowym utratę środków w ramach bardzo nieuczciwego, stronniczego, skrajnie upartyjnionego, jakiego jeszcze nigdy w historii Rzeczypospolitej Polskiej nie było, rozdziału środków koordynowanego przez wojewodów rekomendowanych czy będących w większości politykami Prawa i Sprawiedliwości z tzw. funduszu inicjatyw lokalnych.

Do nich należy m.in. wymiana pieców gazowych w gminie Dzierżoniów albo np. przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej z przeznaczeniem na przedszkole w gminie Szczytna. Tych wniosków jest łącznie ponad 30.

Dziękuję serdecznie, panie pośle.

Wysoki Sejmie! My tutaj je analizujemy, dyskutujemy, natomiast poza tymi tabelami jest jeszcze coś takiego jak klimat toczącej się debaty budżetowej i sygnały, które trafiają do obywateli. Ten klimat jest niestety niewesoły i nie może być inny. W ostatnich dniach obiegła nas informacja, że jeden z restauratorów, który odremontował zabytkowe obiekty i prowadził szanowaną w swoim mieście działalność, powiesił się we własnej, świeżo wyremontowanej sali. Dlaczego? Dlatego że stracił nadzieję. Wielu ludzi w Polsce traci nadzieję, mimo że rząd zrealizuje budżet w przyszłym roku, w najgorszym wypadku go nowelizując. Tak jest zawsze. A dlaczego ludzie tracą nadzieję? Dlatego że nie widzą żadnej racjonalności w tym, co rząd robi, i widzą, że recepta rządu na kryzys to dokręcanie śruby podatkowej. Mówili o tym moi przedmówcy, powtórzę i ja: wprowadzanie nowych podatków w czasach kryzysu to gospodarcze samobójstwo. To wyraz desperacji tego rządu, który pokazuje, że nie ma innego pomysłu na spięcie budżetu niż zabieranie pieniędzy pod coraz to nowymi tytułami. A jeżeli chodzi o te tabele, to czy w ogóle ta nasza debata jest poważna i ma sens, jeżeli w tym roku cała polityka COVID-owa rządu została zrealizowana przez pozabudżetowy fundusz idący w ok. 100 mld zł? Czy my na tej sali, zanim ten fundusz zaczął być realizowany, mieliśmy jakąkolwiek debatę na ten temat? Nie mieliśmy.

Teoretycznie wydatki funduszu COVID-owego nie powiększają długu publicznego, nie są wydatkami publicznymi, zostały schowane w BGK, ale trafiają na Fundusz Pracy czy do ZUS-u, więc już wiadomo, że Unia Europejska policzy nasz faktyczny dług, nasz faktyczny deficyt w inny sposób. A więc debata, którą my tutaj prowadzimy, dotyczy zaledwie wycinka finansów publicznych, i to tego mniej istotnego, tego sztywnego. Tam gdzie rząd sobie zostawia elastyczność, tam jest to poza budżetem państwa. Ten proces już dawno został przez ekonomistów zauważony, nazwany debudżetyzacją finansów państwa. Rząd PiS tutaj twórczo rozwija podstawy i podwaliny pod kreatywną księgowość budżetową, które swego czasu położył minister Jan Vincent-Rostowski z opozycyjnej w tej chwili Platformy Obywatelskiej. Ukrywacie przed obywatelami i przed posłami swoje faktyczne zadania, swoje faktyczne plany i swoje faktyczne działania.

Trzeba wam to mówić prosto w oczy i będziemy wam to mówić. Dziękuję serdecznie. Proszę, panie pośle.

Wtedy, jak mówiliśmy, że jest to oczywiście pusta propaganda, to śmialiście się, pukaliście się w czoło i mówiliście, że nie mamy pojęcia i jeszcze przede wszystkim nigdy nie rządziliśmy, a wy przecież jesteście w tym profesjonalistami. Tak jak mój poprzednik, poseł Bosak powiedział: to jest czysta propaganda, okłamujecie ludzi. Zwyczajnie trzeba wam to pokazywać. Co robicie? Te tarcze antykryzysowe robicie na bazie: widzi nam się, wydaje nam się, tak to pewnie powinno być. Tymczasem drobni przedsiębiorcy niestety na tym cierpią. Jeden z waszych ministrów w jednym z wywiadów powiedział, że rząd radzi sobie z koronakryzysem fenomenalnie. Bardzo bym chciał, żeby to zabrzmiało, ponieważ myślę, że ludzie, którzy nas dzisiaj oglądają, przynajmniej ta część, której zakazaliście pracować, ta część, której zamknęliście firmy, ta część, która zastanawia się, jak powiązać koniec z końcem, ta, dla której nadchodzące święta nie będą zbyt wesołe. Albo jeszcze gorzej: chodzi o tych ludzi, którzy zachorowali - zachorowali nie na koronawirusa, złapali inne choroby i te inne choroby wpędziły ich do grobu.

Za to wszystko odpowiadacie. Tymczasem wasz minister mówi bezczelnie, że wy sobie radzicie fenomenalnie. To jest niestety wasz problem, że w ten sposób (Dzwonek) komunikujecie się ze społeczeństwem. Dziękuję, panie pośle. Przechodzimy do zadawania pytań. Ustalam czas zadania pytania na 1 minutę. Zapraszam pana posła Pawła Rychlika z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość do zabrania głosu. W związku z tym nie kłóćcie się o czas. Prowadzę obrady. Ale to mnie nie mobilizuje, to tylko traktuję jako miłość skierowaną do marszałka. Dziękuję posłankom i posłom za to. Czy pan poseł Paweł Rychlik jest na sali? O, już się skróciło.

Zrobię to z miłością. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Należy rozpatrywać łącznie znowelizowany budżet na 2020 r. i projekt budżetu na 2021 r., bo te budżety się ze sobą ściśle łączą. Rząd wyprowadził poprzez fundusze celowe miliardy złotych polskich podatników, pieniędzy publicznych poza budżet po to, by po pierwsze, manipulować poziomem zadłużenia, manipulować opinią publiczną, a także po to, by poza kontrolą Sejmu - podkreślam - dzielić je dla swoich bez żadnych kryteriów. Ostatni podział na inwestycje lokalne to w pełni potwierdza. Dostały bogate gminy, natomiast biedne, najbiedniejsze otrzymały zero. Moje pytanie: Ile pozostało pieniędzy publicznych na funduszach celowych i jak będą one dalej dzielone? Nikt tego nie wie, proszę państwa. Ostatnie pytanie, które muszę tutaj zadać. Program rozwoju czytelnictwa. Dlaczego w budżecie nie ma ani jednej złotówki na ten program? Czy dlatego że maleje w stopniu zastraszającym poziom czytelnictwa w Polsce? Czy mamy doprowadzić do tego, że nikt już nie będzie czytał, bo nie ma w bibliotekach nic do czytania, żadnych nowości? Pani posłanka Katarzyna Kretkowska z klubu parlamentarnego Lewica. Będziemy się łączyli zdalnie z panią posłanką.

W tej chwili ona wynosi niecałe 55% środków potrzebnych na utrzymanie szkół i zjada całkowicie środki bieżące samorządów, które są potrzebne na inne cele związane bezpośrednio z życiem codziennym ludzi, takie cele jak ośrodki zdrowia, usługi opiekuńcze, usługi socjalne, żłobki, utrzymanie porządku, bezpieczeństwa, dróg etc.

Budynek po dworcu Poznań Główny stoi pusty, jest to piękny zabytkowy budynek. Natomiast dworzec został przeniesiony do centrum handlowego i jest tam na zasadzie prawa kaduka, w tym centrum handlowym jest zupełnie niepraktyczny, jest źródłem irytacji, a nie komfortu podróżnych.

Ten budynek został zabrany przez Kościół i szkoła muzyczna nie ma swojego budynku. Miasto przeznaczyło dla tej szkoły muzycznej działkę pod. w budżecie państwa znalazły się środki na rozpoczęcie budowy tej szkoły. Dziękuję bardzo. Dziękuję za głos. Oddaję głos panu Krzysztofowi Paszykowi, Klub Parlamentarny Koalicja Polska. Proszę bardzo. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Trzy krótkie pytania.

Dlaczego nie ma środków na wypłatę trzynastej emerytury? Dlaczego nie ma środków na program leki dla seniorów 75+? Dlaczego nie ma funduszu modernizacji placówek służby zdrowia? To są trzy fundamentalne pytania. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Zapraszam pana posła Krystiana Kamińskiego, koło Konfederacja. Wysoka Izbo! Mamy bardzo optymistyczne założenia budżetowe - ogromny wzrost PKB w przyszłym roku. Tylko kto ma ten wzrost wypracować? Obłożyliście podwójnym podatkiem spółki komandytowe, które w związku z tym nie będą pracować w takiej formie - ponad 40 tys. spółek, 3 mln zatrudnionych. Zarżnęliście gastronomię, zarżnęliście branżę fitness. Kto ma ten wzrost wypracować? Pomimo takiego wzrostu założyliście 82 mld długu. W związku z tym mam pytanie: Kto i kiedy spłaci ten dług? Na pewno nie wasz rząd, prawdopodobnie będzie musiał to zrobić rząd Konfederacji. Dziękuję serdecznie za ten pełen nadziei głos, panie pośle. Pani posłanka Agnieszka Ścigaj, niezrzeszona. Zapraszam serdecznie. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Budżet to też budżet przeciętnego Polaka.

Badanie po wirusie pokazuje również to, jak spadnie siła nabywcza Polaków. Ten budżet to budżet potężnego długu, o którym tak naprawdę jeszcze do końca nie wiemy, jaki jest. Ponieważ państwo wyłączyliście spod reguły wydatkowej inwestycje, o których mówił pan minister, do końca nie będziemy wiedzieć, jaki dług zostawiamy nowemu pokoleniu. 70% młodych Polaków chce wyjechać. Co w tym budżecie jest dla tych Polaków? Co spowoduje, że ich zatrzymamy? To oni będą musieli pracować na długi. Dziękuję serdecznie. No ale zobaczymy.

Wysoka Izbo!

Mam pytanie do pana ministra. Czy przedstawione rzekome podatki mają rzeczywiście charakter fiskalny i można je nazwać podatkami, np. opłatę retencyjną?

Dziękuję bardzo. Pewnie odpowie na to pytanie pan poseł Aleksander Miszalski z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Chciałbym zapytać rządzących, czy mogliby wreszcie przeznaczać pieniądze zbierane od Polaków na sprawy, które są ważne dla naszych rodaków i potrzebne, zamiast na PiS-owską propagandę, na wynagrodzenia dla swoich partyjnych kolegów oraz na instytucje współpracujące politycznie? Wydajecie na infrastrukturę kolejową zaledwie 900 mln zł, ale na TVP - 2 mld, na rzecznika praw obywatelskich - 50 mln zł, ale na radę radiofonii i telewizji - ponad 63, na Polską Akademię Nauk - 91 mln zł, ale na Fundusz Kościelny - 140, na lecznictwo psychiatryczne - 87, ale na IPN - 400 mln.

Dziękuję bardzo, panie pośle. Pan poseł Marek Rutka, klub parlamentarny Lewica. Zapraszam. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Klub parlamentarny Lewica od samego początku za jeden ze swoich priorytetów uznaje poprawę stanu zdrowia Polek i Polaków. Szacuje się, że endometrioza, czyli ciężkie schorzenie ginekologiczne, dotyka 300 mln kobiet na świecie. W Polsce z tą chorobą zmaga się nawet 2 mln kobiet. Dlatego jako przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Endometriozy chciałbym zapytać, czy rząd Prawa i Sprawiedliwości poprze poprawkę mojego autorstwa oznaczoną nr 262, która zakłada zwiększenie o 30 mln zł kwoty, która ma być przeznaczona na stworzenie krajowego programu badań profilaktycznych i skutecznego leczenia endometriozy. Warto podkreślić, że wysokość refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia za zabieg usunięcia zmian w obrębie jajników, czyli tzw. endometriozy jajników, wynosi 2100 zł, a realny koszt zabiegu, który pacjentki zmuszone są pokrywać z własnych pieniędzy, z własnej kieszeni, wynosi ponad 20 tys. zł. Dziękuję serdecznie. Proszę bardzo. Wysoka Izbo!

Chodzi przede wszystkim o brak na liście budowy bloku operacyjnego w szpitalu w Rawie Mazowieckiej. Jakie to kryteria państwu przyświecały, że budowa parkingu przy gminie wygrała, jest na liście, a nie ma tak ważnej inwestycji jak remont, budowa bloku operacyjnego w szpitalu? Mam także pytanie o inwestycje, na które bardzo długo czekają mieszkańcy województwa łódzkiego: Czy powstanie wreszcie droga S14 z obwodnicą Sulejowa, którą obiecywali politycy PiS-u przed wszystkimi wyborami, które miały miejsce ostatnio? Czy zostanie wybudowana obwodnica Skierniewic wraz z miejscowością Mokra Prawa? Czy wreszcie powstanie przystanek kolejowy w miejscowości Żurawia w powiecie (Dzwonek) rawskim, o który zabiegają samorządowcy z powiatu rawskiego, z wszystkich okolicznych gmin? Bardzo proszę o odpowiedź na te pytania. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. W związku z tym poproszę pana posła Mirosława Suchonia z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska.

Bardzo dziękuję, panie marszałku, również za to doprowadzenie do mównicy, bo sprawa rzeczywiście ważna. Wysoka Izbo! Tak twierdzili przedstawiciele rządu, ale do spełnienia tych deklaracji zabrakło rzeczy podstawowej - dobrego budżetu. Dlatego zgłaszam do budżetu ponad 20 zmian, które budżet z punktu widzenia m.in. mieszkańców Bielska Białej, powiatu bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego i żywieckiego poprawiają. I te środki finansowe to ponad 115 mln zł dla szpitali, także 100 mln zł na walkę ze smogiem na południu województwa śląskiego, kolejna grupa to 800 mln zł na infrastrukturę, m.in. na Beskidzką Drogę Integracyjną oraz skrzyżowania w Ustroniu, w Pszczynie, w Czechowicach-Dziedzicach. Ale też zgłaszam (Dzwonek) poprawkę dotycząca edukacji ekonomicznej. Myślę, że to jest bardzo ważna poprawka. I proszę rząd o to, aby odpowiedział, czy jest skłonny poprzeć tę poprawkę. Otóż jest to program edukacji ekonomicznej dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, który ma spowodować, aby młodzież potrafiła odróżnić kłamstwo, propagandę rządu Prawa i Sprawiedliwości, od prawdy i rzeczywistości. I pytanie: Czy rząd jest skłonny poprzeć tę dobrą poprawkę? No na pewno, panie pośle. Proszę bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Nieobecny Panie Ministrze! Usłyszeliśmy dziś: rząd Zjednoczonej Prawicy uważa, że przygotował budżet bezpieczeństwa i budżet inwestycji. To ja pytam: Jak bezpiecznie mają się czuć osoby pracujące w służbie zdrowia, jak mają się czuć pacjentki i pacjenci szpitali niejednokrotnie stojących na krawędzi wydolności finansowej, bez środków na inwestycje, bez środków na leczenie? Jak mają się czuć emeryci, seniorzy, którzy zostali pozbawieni trzynastej emerytury? Bo co, bo nie ma roku wyborczego? Jak mają się czuć mieszkanki i mieszkańcy samorządów, patrząc, jak rząd przeprowadził podział funduszy wsparcia według kryteriów politycznych, a nie potrzeb społeczności lokalnych? Jak mają się czuć regiony Warmii i Mazur, Powiśla, takie miejscowości jak Iława, Elbląg, Olsztyn, Ełk pozbawione inwestycji, o które zabiegają, by wyrównać standardy życia z innymi regionami Polski [[Dzwonek]] czy Europy? Dziękuję serdecznie. Pan poseł Andrzej Grzyb, Klub Parlamentarny Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści. Proszę bardzo. Wysoka Izbo! Od paru debat próbuję dociekać, dlaczego to od 2015 r. sukcesywnie co roku spadają nakłady na rolnictwo.

Jednocześnie mamy oczywiście też taki wskaźnik, który mówi, że powinien ten wskaźnik wynosić gdzieś ok. 1%, jeżeli chodzi o PKB.

Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Nie ma pana posła Michała Urbaniaka. A więc pan poseł Krzysztof Piątkowski, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Proszę bardzo. Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Najważniejsza debata trwa w Sejmie, a nie ma ministra, nie ma premiera. Może dobrze, że nie ma pana premiera, bo pewnie mówiłby, jaki to znakomity budżet, jak jest świetnie w Polsce, a ilekroć mówi „dobrze”, to okazuje się, że jest jeszcze gorzej, niż wszyscy myśleliśmy.

Po raz kolejny planowany wzrost subwencji oświatowej nie będzie nadążał za wydatkami na oświatę, a w znaczącym stopniu to właśnie ten rząd odpowiada za te wydatki. W większości te dochody spadły z powodu braku decyzji [[Dzwonek]] albo złych decyzji obecnego rządu. Dziękuję serdecznie. Pani posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, klub parlamentarny Lewica. Nie ma pani posłanki.

Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe, unia demokratów, Konserwatyści. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Tutaj przed chwilą mój kolega klubowy już pytał o to, ale to jest bardzo ważna kwestia.

I wy ciągle powtarzacie, że my nie dbaliśmy w poprzedniej koalicji o rolnictwo. Z drugiej strony jest coraz więcej wyzwań: ta piątka, o której tu dyskutowaliśmy, za chwilę wchodzi nowy zielony ład. Nie przygotowujecie w żaden sposób rolników.

Dziękuję serdecznie. Pan poseł Artur Dziambor, koło Konfederacja.

Panie pośle, proszę bardzo. W imieniu mojego kolegi posła Urbaniaka dziękuję bardzo za tę decyzję. Ja dalej o podatkach, ponieważ premier Morawiecki powiedział, że podatki, które są teraz podnoszone, to są podatki, które będą zbierane po to, żeby ratować to, co zostało po koronawirusie, żeby pomóc jakoś społeczeństwu, ponieważ wiadomo, że trzeba jakoś sobie radzić z tymi wypłatami z tarcz. Minister finansów. Jak on się nazywał? Minister finansów, który tutaj czasem rzeczywiście wpada, ale jakoś rzadko się wypowiada, wysługuje się swoim młodym zastępcą, który co wywiad strzela jakieś kompletne gafy. Tak że wracam do mojej pierwszej wypowiedzi. Przy tym poziomie państwa samozadowolenia i bezczelności trudno przewidzieć, co nam jeszcze planujecie, ale bardzo chciałbym usłyszeć, jakie podatki planujecie podnosić od stycznia, bo jak wiemy, od początku tej kadencji co miesiąc coś nowego wprowadzacie. Czy pan poseł Cezary Grabarczyk jest na sali? Nie ma. Zapraszam pana posła Krzysztofa Śmiszka, klub parlamentarny Lewica. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 2020 r. to rok, który odcisnął się koszmarnym piętnem na sytuacji wielu grup społecznych, a także zawodowych. Jedną z nich, mam wrażenie, że zupełnie zapomnianą i o której w ogóle się nie dyskutowało, są pracownicy polskich sądów. Zbyt często zapominamy o tych, dzięki którym sądy, polskie sądy ciągle mogą pracować niezależnie. Niezależnie przede wszystkim od prób nacisków i upolityczniania. Asystenci, referendarze, kuratorzy, protokolanci - to oni na co dzień służą Polkom i Polakom, niewidoczni, pracujący za śmieszne pieniądze. Chcę zapytać, jak rząd ocenia ich poziom wynagrodzenia i jakie plany ma rząd na ich [[Dzwonek]] przyszłość finansową i zawodową. Złożyłem poprawkę przyznającą administracji sądowej po 300 zł brutto. Zasługują oni na to, aby mieć wyższe wynagrodzenia.

Nadzieja zwykle umiera ostatnia. Pan poseł Marek Sawicki, Klub Parlamentarny Koalicja Polska, tym razem Polskie Stronnictwo Ludowe. Proszę bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Nieobecny Panie Premierze! Chwalicie się państwo, że ten budżet jest zasobny, a ja martwię się, że tych pieniędzy, które macie w tej chwili, nie potraficie zagospodarować i racjonalnie wydać. Zaległości w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Chcę także zapytać, czy skończycie z tym marnotrawstwem w Krajowym Ośrodku Wparcia Rolnictwa. A jednocześnie wynajmujecie siedzibę na ul. Karolkowej, [[Dzwonek]] bo rzekomo jest wygodniejsza dla dyrektora generalnego. Połączymy się z panem posłem Korwin-Mikkem, z którym nie mogliśmy się połączyć. Jest. Proszę bardzo, panie pośle.

Jakby pan mikrofon włączył, panie pośle. Wysoka Izbo!

A więc im mniejszy budżet, tym lepiej.

Proszę państwa, ciężko mi rozmawiać z politykami, którzy nie rozumieją elementarza ekonomii. Dziękuję za uwagę. Dziękuję serdecznie. Proszę bardzo. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W wasz epokowy „Program dla Śląska”, który miał zmienić oblicze naszego regionu, nie wierzy już chyba nikt. Nawet sprzymierzony z wami szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” powiedział ostatnio, że „Program dla Śląska” pachnie jak spalony kotlet i podobnie wygląda. Kiedyś pewnie powstanie muzeum obietnic Mateusza Morawieckiego i tam „Program dla Śląska” będzie stał pomiędzy promem Batory, stutysięcznym mieszkaniem a milionowym elektrykiem na polskich drogach. Zapewne w odpowiedzi usłyszę, że miliardy są zaangażowane i pracują, ale nie usłyszę, co to znaczy, że te środki są zaangażowane i pracują. A może ktoś mnie i moje koleżanki i partyjnych kolegów określi mianem członków ugrupowania z zewnątrz, co, między nami mówiąc, jest podłością. Moje pytania: Ile środków zapewniają państwo na realizację „Programu dla Śląska” w 2021 r. Kiedy odtajnicie protokoły Komitetu Sterującego i Rady Wykonawczej „Programu dla Śląska” Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Od lat parki narodowe, nasz skarb narodowy, wskazują najważniejszą barierę rozwoju, czyli brak funduszy. Parki krajobrazowe są wręcz tragicznie niedofinansowane i bez finansowania, bez tych środków nie są w stanie wypełniać jakichkolwiek zadań. Zachowanie i poszerzanie tych parków jest kluczowe dla naszej przyszłości, bo jest to element walki z katastrofą klimatyczną. Te obszary są także kluczowe dla kwestii powodzi i suszy, dla gospodarki wodnej. Ich wpływu nie da się przecenić. Za to, jak widać, rząd ceni je zdecydowanie mniej - widzimy to w tej propozycji budżetowej. Woli wycinać lasy, proponując ustawę o drewnie energetycznym, niż zachowywać to, co jest najcenniejsze. Konieczna jest zmiana priorytetów. W jaki sposób tak niedofinansowane parki mają prowadzić działania ochronne wobec ekosystemów? Jak zespoły parków krajobrazowych mają przy tak małym finansowaniu funkcjonować sprawnie? Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Proszę bardzo. Wysoka Izbo! Nieobecny Ministrze Finansów!

Dwa tematy. Drogi lokalne. Jestem z Pomorza Zachodniego. 15 tys. km dróg lokalnych, czyli tych gminnych i powiatowych. 100 lat, 150 lat chcemy to budować? Drugi temat. Drogi rządzie, przestańcie wreszcie oszukiwać, a przede wszystkim ograbiać polskie samorządy. Nie płacicie określonej subwencji oświatowej, samorządy dopłacają ze swoich pieniędzy. Szanowni państwo, to jest zadanie państwa. Dziękuję serdecznie. Proszę państwa, mam taką refleksję jednozdaniową. Mam prośbę do opozycji, żeby przestała atakować rząd w sposób bezmyślny. Pan minister finansów przecież nie musi być na obradach wtedy, kiedy rozmawiamy o budżecie. To nie są sprawy, które są najważniejsze dla ministra finansów. Są widocznie inne, ważniejsze sprawy, o których nie wiecie. Tak że bardzo proszę, naprawdę, bez takich cynicznych, ironicznych uwag. Bardzo proszę. Pan poseł Arkadiusz Marchewka, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Taka jest prawda o finansach państwa. Tymczasem co mówi premier Morawiecki? Premier Morawiecki ostatnio z tej mównicy stwierdził, że dzięki determinacji Jarosława Kaczyńskiego finanse publiczne są w tak dobrym stanie jak nigdy. Obiecywaliście zrównoważony budżet, a zamiast tego jest rekordowa dziura. Tę dziurę chcecie zasypać pieniędzmi z portfeli obywateli, nakładacie więc nowe podatki: podatek cukrowy, podatek handlowy, wyższą opłatę mocową, czyli wyższe opłaty za prąd, CIT dla spółek komandytowych, firm rodzinnych, [[Dzwonek]] likwidację ulgi abolicyjnej dla osób pracujących za granicą, a pewnie niedługo podatek od deszczu. To jest nieodpowiedzialne zarządzanie finansami publicznymi, a wy nie powinniście swoich błędów przelewać na obywateli, bo to nie obywatele są temu winni, więc te podatki są niesłuszne. Powinniście bardziej zajmować się i martwić się tym, jak tę dziurę ograniczać, a nie spychać to na obywateli. Dziękuję serdecznie. Pan poseł Marchewka dostał brawa za to, że był przeciwko podatkowi od deszczu. Pani posłanka Paulina Matysiak z klubu parlamentarnego Lewica. Zapraszam. Jesteśmy ciekawi pytania. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dzisiaj odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa poświęcone sytuacji składowisk odpadów w Gorlicach i Zgierzu. Oczywiście to nie jest tak, że mamy tylko te dwa składowiska odpadów, problem jest szerszy i dotyczy całej Polski.

Sytuacja jest zła, by nie powiedzieć: tragiczna. Czy nie jest to właściwy moment, żeby poszukać pieniędzy na to, żebyśmy posprzątali wreszcie Polskę, tak byśmy mogli żyć i mieszkać w bezpiecznym kraju? Dziękuję serdecznie. Pan poseł Jan Łopata, Koalicja Polska. Dobra. Pan poseł Tomasz Olichwer, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

To jest jedno pytanie. Drugie pytanie. W jaki sposób macie zamiar zrekompensować te krzywdzące decyzje podjęte w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z którymi wiele gmin takich jak Dąbrowa Mogileńska, Kcynia, Inowrocław, Strzelno, Mogilno nie otrzymało żadnych środków finansowych. Trzeba ten błąd naprawić i skończyć z partyjnym rozdzielaniem pieniędzy.

Kultura wymaga, żeby te przeprosiny przyjąć, więc w imieniu przeproszonych dziękuję za te przeprosiny. Pan poseł Michał Szczerba, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Szanowny Panie Marszałku! Za Warszawę nie będziemy przepraszać, o Warszawie będziemy mówić, bo trzeba mówić, ponieważ epidemia trwa, a rząd coraz głębiej sięga do kieszeni samorządów, chce podzielić Mazowsze i odciąć je od niektórych funduszy unijnych. W wyniku jego wadliwej konstrukcji, pomimo znacznego ubytku dochodów i w tym roku, i w przyszłym, Warszawa w przyszłym roku ma zapłacić 1300 mln zł, tj. o 85 mln zł więcej niż w tym roku. Potrzebne są zatem środki na takie inwestycje, jak budowa Sinfonia Varsovia Centrum przy ul. Grochowskiej, zadaszenie Toru Łyżwiarskiego Stegny, budowa hali widowiskowo-sportowej przy stadionie i wreszcie rozpoczęcie budowy stadionu lekkoatletycznego Skry.

Zamiast pieniędzy na pamięć narodową, na zwiększanie pensji coraz większej grupy urzędników przekażmy 10 mln zł na rozpoczęcie programu dla chorych na choroby otępienne, na chorobę Alzheimera w naszym kraju. To będzie dobry uczynek Wysokiej Izby, który możecie zrobić w przyszłym roku. Dziękuję serdecznie.

Dziękuję, panie marszałku. Na skutek odmowy sfinansowania wielu sensownych, potrzebnych, pożytecznych projektów z funduszu inicjatyw lokalnych dziesiątki gmin na Dolnym Śląsku zostanie pozbawionych dofinansowania. W imieniu niektórych z nich zwróciłem się z poprawkami.

Dotyczą one również kwestii ekologicznych, jak chociażby obudowy instalacją fotowoltaiczną budynków użyteczności publicznej w gminie Warta Bolesławiecka. Są tam inwestycje innowacyjne, takie jak budowa w Bielawie inkubatora art-przedsiębiorczości.

Wreszcie są też takie, które dotyczą edukacji, bardzo ważnej dziedziny, np. modernizacja szkoły podstawowej w gminie Pęcław czy przebudowa, rozbudowa budynku szkoły podstawowej na użytek przedszkolny w miejscowości Szczytna. I te wszystkie inwestycje proponuję sfinansować nie z powiększenia długu publicznego, tylko właśnie ze zmniejszenia długu publicznego, z obniżenia kosztów pożyczenia pieniędzy przez rząd polski, zwłaszcza że na skutek przyjęcia Funduszu Odbudowy w Unii Europejskiej takie pożyczanie na cele walki ze skutkami COVID będzie tańsze, koszt tego będzie niższy, niż gdybyśmy ten Fundusz Odbudowy odrzucili. Dziękuję serdecznie. Proszę, panie pośle. Dziękuję. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ten budżet to budżet pobożnych życzeń działaczy PiS i dla działaczy PiS. Płaci działaczom PiS i tam, gdzie oni rządzą, a tam, gdzie nie rządzą - nie płaci. I tak nie dociepla domów pomocy społecznej w Łodzi, bo nie rządzi w Łodzi nikt z PiS. Nie remontuje budynku, gdzie mieszkają ludzie w Kutnie, bo w Kutnie też nie rządzi. Ale do historii przejdzie budowa obwodnicy Łodzi, gdzie nie będzie zjazdu do miasta Łodzi, bo właśnie w Łodzi PiS nie rządzi. Jest. Jest. Wszystko bezzwrotnie. Jest. Jest. 250 mln zł dla ojca Rydzyka?

Dziękuję serdecznie, panie pośle. Pani poseł Marta Wcisło, Koalicja Obywatelska. Proszę bardzo. Wysoka Izbo! Do was nic nie dociera, bo nie ma do kogo.

Jedyne, co umiecie, to szastać publiczną kasą. Szanowni Państwo! Co jest priorytetem dla rządu w nowym roku? 200 mln więcej na kancelarię premiera. Nowe limuzyny dla rządu, których będzie więcej niż karetek w Polsce. Szanowni państwo, czy to naprawdę powinny być priorytety rządu w czasie kryzysu i epidemii? Dlaczego nie chcecie dać pieniędzy na Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, na centrum zdrowia seniora w Lublinie czy na centrum wsparcia rodziny, skoro prowadzicie politykę prorodzinną? O to wszystko proszę. Apeluję do posłów z regionu, aby poparli wnioski regionalne.

Szanowni państwo, obecny rząd jest niestety ekonomicznym analfabetą. Dziękuję serdecznie. Zapraszam panią poseł Paulinę Hennig-Kloskę, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Mimo epidemii, mimo kryzysu gospodarczego ceny w Polsce nadal szaleją. Inflacja w Polsce jest najwyższa w całej Unii Europejskiej. Wam jednak wciąż mało i na przyszły rok ponownie fundujecie nam szereg impulsów inflacyjnych, które będą powodowały dalszy wzrost cen. Tak jest co roku, dlatego od lat mamy inflację najwyższą bądź jedną z najwyższych w Europie. Mieliśmy już takie przypadki. Opłata od wymiany oleju sprawi, że użytkowanie naszych aut będzie po prostu droższe.

Bardzo proszę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Nie lubicie, ponieważ warszawiacy i warszawianki was nie popierają, a prezes Kaczyński powiedział jasno: proszę nas popierać i nie przeszkadzać. I wszyscy ci, którzy się temu sprzeciwiają, nie wypełniają tej prośby, płacą za to wysoką cenę. Swoją niechęć do warszawianek i warszawiaków pokazujecie w różny sposób: fizycznie, pacyfikując strajki na ulicach stolicy, ale też finansowo, zabierając warszawiakom szansę na potrzebne dla ich rozwoju inwestycje. Ostatnio pominęliście nas w funduszu inwestycji lokalnych. Mam nadzieję, że zdajecie państwo sobie sprawę z tego, że wy nie pomijacie samorządu, którego nie lubicie, polityka, którego nie lubicie, tylko pomijacie mieszkańców, [[Dzwonek]] którzy czekają na nowe placówki medyczne, przedszkola, żłobki i szkoły. I z racji tego, że w tym budżecie też nie pojawiają się dobre dla Warszawy punkty budżetowe, złożyłam szereg poprawek - od dofinansowania Szpitali: Południowego, Praskiego i Wolskiego po budowę żłobków, linii tramwajowych na Tarchomin czy zakup niskoemisyjnych autobusów. Macie państwo jeszcze szansę zrobić coś dobrego dla mieszkańców Warszawy. Chciałabym, żebyście oddali im pieniądze, wsparli ich w potrzebnych im inwestycjach. Niech nie będą ofiarami waszej politycznej zemsty. Dziękuję serdecznie. Pan poseł Marek Sowa, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Kolejny budżet, w którym zadłużacie Polskę na kolejne 135 mld zł. Do tego 10 nowych podatków. Kolejne ich podwyższanie w waszym wykonaniu nie ma już po prostu końca. Wydawałoby się, że po takich ruchach w tym budżecie kasa będzie na wszystko, że starczy na wszystko. Niestety nic z tego, Polacy z tego nic nie mają. W imieniu mieszkańców Małopolski złożyłem kilkanaście poprawek do tego budżetu, bo ostatnio, w ubiegłym tygodniu zostali brutalnie przez Mateusza Morawieckiego i polityków PiS-u okradzeni. 2 mln Małopolan zostało bez grosza wsparcia. W tym budżecie macie ostatnią szansę, aby jeszcze zagłosować za poprawkami, które wesprą małopolskie szpitale, pozwolą dokończyć rozbudowę szpitala uniwersyteckiego, pozwolą zakończyć budowę specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, o którym tak często mówicie, że jest bardzo potrzebny i powinien zostać zrealizowany.

Chcecie brać, a właściwie kraść z tego budżetu, ile się da. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę. Po pierwsze, powinniśmy żądać tego, aby na tej sali w tej dyskusji brał udział minister finansów. To jest kluczowa debata o finansach. Państwo zadłużyliście nasz kraj na blisko 600 mld zł w ciągu ostatnich kilku lat. I dzisiaj, kiedy mówimy o budżecie, także o wszystkich ważnych elementach regionalnych, chciałbym powiedzieć o kilku z nich.

Sąsiednie powiaty po 20, 30 mln. Dlatego wnoszę o to, aby obwodnica Złotoryi była finansowana z tych środków.

To jest budżet ostatniej szansy dla gmin, którym de facto odebraliście finansowanie z funduszu inicjatyw lokalnych. To jest moment na to, żebyście przyjęli nasze poprawki. Dziękuję serdecznie. Pan poseł Krzysztof Gadowski, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Nie ma ministra, więc skieruję ten wniosek na ręce obecnych tu pracowników ministerstwa. W 2016 r. zamroziliście projekt, który gwarantował ochotnikom strażakom dofinansowanie do emerytury.

Chciałbym się zapytać, w jaki sposób zrealizujecie tę obietnicę. W poprawce do budżetu skierowałem kwotę 50 mln zł na ten cel. Czy rząd poprze tę poprawkę, czy ma jakiś inny pomysł na to, żeby ta dopłata do emerytury dla ochotników strażaków się pojawiła? W jaki sposób chcecie wspomóc samorządy na Śląsku w rewitalizacji zdegradowanych terenów górniczych, gdzie są potężne dziury, pocięte zawaliska, tereny, które są zniszczone? W jaki sposób chcecie wspierać samorządy w budowie i modernizacji dróg na Śląsku? Mówię o głównej drodze, drodze południowej w powiecie wodzisławskim, o drodze regionalnej Racibórz - Pszczyna w Rybniku i odcinku wiodącym do Raciborza. W jaki sposób chcecie wesprzeć te samorządy? Czy macie pomysł?

Czy w tym budżecie państwa macie zapisane te środki, czy nie?

Bardzo proszę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jeszcze nie tak dawno, bo w środę, premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska ma dzisiaj finanse publiczne w tak dobrym stanie jak nigdy w historii. Jeżeli jest to prawdą, to podkarpackie inwestycje powinny być zrealizowane w szybkim czasie. Poprawki przeze mnie zgłoszone to poprawki bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju regionu. Jest to droga ekspresowa, łącznica kolejowa, zjazdy z autostrady i wiele, wiele innych bardzo ważnych inwestycji. Szanowni Państwo! Nie sztuką jest podpisywać listy intencyjne. Sztuką jest zrealizować obietnice. Apeluję teraz do posła Marka Kuchcińskiego, aby zobowiązał posłów Zjednoczonej Prawicy, jeśli chodzi o głosowanie za przyjęciem tych poprawek. Jeżeli zagłosujecie państwo za przyjęciem tych poprawek, wtedy uwierzę premierowi, [[Dzwonek]] że w środę mówił prawdę. Po czynach was poznamy. Dziękuję serdecznie. Zapraszam bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Gdy zsumujemy te liczby, wyjdzie nam 8 mln osób, obywateli. Szanowni państwo, tej liczby nie można zignorować, bo to jest poważny problem ilościowy i jakościowy dla całego systemu opieki zdrowotnej. Szanowni Państwo! Co najbardziej bulwersuje cukrzyków w naszym kraju?

Należy doprowadzić do wyrównania dostępu do nowoczesnych terapii cukrzycowych (Dzwonek) dla wszystkich pacjentów diabetologicznych. Należy również przeprowadzić ogólnopolską kampanię społeczną mającą na celu uświadomienie społeczeństwu, jak podstępną i groźną chorobą jest cukrzyca, która często spowodowana jest złą dietą, skutkującą początkowo otyłością, a następnie poważnymi powikłaniami sercowo-naczyniowymi, również wieloma innymi przykrymi powikłaniami, natomiast ostatecznie nieleczona prowadzi do przedwczesnych zgonów. Szanowny panie ministrze, wiceministrze, bo pana ministra nie ma, bardzo serdecznie proszę w imieniu Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy o uwzględnienie tych dwóch poprawek. To jest palący, pilny problem, który musi być uwzględniony w tym budżecie. Proszę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jest faktycznie rzeczą zaskakującą, że debata o kształcie budżetu na przyszły rok cieszy się tak małym zainteresowaniem ze strony posłów partii rządzącej, bo to dziś powinniśmy ustalić najważniejsze kryteria wydatkowania środków publicznych. Chcę na dwie rzeczy zwrócić dziś państwa uwagę. Jest rzeczą dramatyczną, jak słucha się samorządowców, którzy nie są w stanie wybudować przedszkola we własnej gminie, dlatego że rząd rozdziela pieniądze według sympatii politycznych. Chciałabym, żeby państwo jeszcze dzisiaj się do tego odnieśli. Natomiast jeśli chodzi o budżet na przyszły rok, mają państwo bardzo dużo poprawek, ale większość z nich jest niezwykle ważna i nic chciałabym widzieć, że lekką ręką odrzucacie je tylko dlatego, że złożyła je opozycja. Proszę zwrócić uwagę na poprawki dotyczące chociażby psychiatrii dziecięcej, tak bardzo potrzebującej dofinansowania w dzisiejszych czasach, i proszę o ich przyjęcie. Zapraszam, pani posłanko. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dług publiczny wynosi obecnie 1300 mld. To są astronomiczne sumy. Dosłownie. A więc pytam: Jak zamierzacie ten astronomiczny dług spłacić? Jakie podatki na nas jeszcze nałożycie? Przypomnę, że przyszłym roku wpływy z podatków spadną o 40 mld, a według raportu Tax Foundation wśród krajów OECD polski system podatkowy jest jednym z najgorszych, trzeci od końca. Jak długo jeszcze będziecie ukrywać wydatki i wyrzucać je poza budżet, w ten sposób omijając próg ostrożnościowy w konstytucji? Ile jeszcze kartek z tej biednej, sponiewieranej przez was konstytucji wyrwiecie, by ukryć swoją nieudolność? Proponuję, by wprowadzić nową miarę zadłużenia i waszą nieudolność mierzyć w galaktykach, bo miliony i miliardy to dla was za mało. Ten rząd musi odejść, zanim doprowadzicie ten kraj do bankructwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pani posłanko. Zapraszam. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chętnie zwróciłbym się do ministra finansów, ale go nie ma. Zwróciłbym się chętnie do wiceministra Patkowskiego, ale też go nie ma. Nie ma parlamentarzystów z ziemi radomskiej. Ale chciałbym zwrócić się do tych, którzy są tu obecni. Przekażcie posłom z Radomia, posłom Prawa i Sprawiedliwości: Warto głosować za poprawkami radomskimi. Warto głosować za poprawką, która da naszemu miastu pieniądze na budowę wiaduktu, wiaduktu tak potrzebnego również ministrowi Weberowi, który tutaj jest z nami, bo jest to wiadukt, który będzie służył lotnisku w Radomiu.

Dopóty dopóki będę posłem (Dzwonek), będę powtarzał: w Pionkach musi być bezpiecznie. Nie może miastu grozić wybuch, który jest pozostałością po czasach słusznie minionych, kiedy to fabryka prochu w Pionkach zostawiła tam odpady. I na koniec, szanowni państwo: epidemia, jakże ważna. Były wojewoda mazowiecki, pewnie przyłączy się do mojego zdania. Szanowni państwo, sprawa karetki w Kozienicach - nie może być tak, że będziemy zabierać karetkę i dawać do innej miejscowości.

Dziękuję serdecznie. Pan poseł Michał Krawczyk, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! O tym, że żyjemy w trudnych czasach, nie musimy się przekonywać. Natomiast musimy przekonywać rząd PiS do tego, w jaki sposób zarządzać finansami państwa i budżetem państwa na przyszły rok w tej trudnej sytuacji, w której jesteśmy w czasie epidemii. Otóż zaskakuje nas podejście rządu, w którym zamiast ograniczać całkowicie niepotrzebne, horrendalne wydatki na megalomańskie inwestycje, wy je państwo kontynuujcie.

W kilka minut w budżecie państwa można znaleźć oszczędności na przyszły rok rzędu 6 mld zł. Natomiast państwo wolicie kontynuować te inwestycje po to, żeby z każdym rokiem wzrastał dług Polski (Dzwonek), który obciąża każdą Polkę i każdego Polaka. Zamiast inwestować w szpitale, wychodzicie z założenia, że nie trzeba tam nic poprawiać, bo wystarczy mówić w TVP, że się poprawia. W zeszłym roku odrzuciliście państwo wszystkie poprawki, które były złożone do budżetu. Mam nadzieję, że w tym roku przynajmniej je przeczytacie, zanim bezmyślnie zagłosujecie przeciw. Dziękuję serdecznie. Myślę, że jak posłowie są nieobecni, to nie wysłuchali pana apelu. Pani poseł Katarzyna Lubnauer, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Co rośnie PiS? Podatki. Większość krajów obniża podatki z powodu kryzysu, natomiast PiS wprowadza osiem nowych podatków. Luka VAT. Chciałoby się spytać: Zaczęliście kraść? Dług publiczny - 600 mld wzrosło, mimo że mieliście ileś lat świetnej koniunktury.

Przynajmniej według waszych statystyk. Inflacja - rekord jeśli chodzi o Unię Europejską w październiku, też wam wzrosła. No i wydatki na telewizję publiczną: na TVPiS, na to szambo wydajecie 2 mld rocznie przez kolejnych 5 lat, od zeszłego roku licząc, właściwie od tego roku licząc, na przyszłość. No i teraz rodzi się jedno pytanie: Gdzie jest autor tego sukcesu, tego, że wszystko rośnie? Pan premier jest nieobecny, [[Dzwonek]] pan minister finansów jest nieobecny, pewnie się wstydzą. Bo okazało się, że podatnicy potrafią omijać prawo i w związku z tym wychodzi na to, że rozpijacie Polaków. Pani posłanka Monika Rosa, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! To nie jest dobry budżet, bo jest w nim sporo wydatków bezsensownych lub szkodliwych jak finansowanie telewizji publicznej. Ale jest także brak finansowania priorytetów jak ochrona zdrowia. Chcę zwrócić uwagę na trzy elementy. Po pierwsze niska emisja. Są konkretne dane, które mówią o tym, że dzieci rozwijające się w zanieczyszczonym powietrzu mają zaburzenia koncentracji, częściej chorują na ADHD, mają schorzenia z grupy autyzmu. Miast, które potrzebują wsparcia w walce z emisją, jest coraz więcej, ale wydatki z budżetu państwa są wciąż za małe. Drugi element: nie widzę w budżecie pieniędzy na to, by wyrównać świadczenia dla opiekunów dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami. To jest wyrok sprzed lat, który wciąż nie jest realizowany. Ta pomoc jest wciąż za mała. Po trzecie, chciałam zapytać o jasne kryteria, [[Dzwonek]] to, w jaki sposób były przydzielane pieniądze w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dziękuję serdecznie. Pan poseł Mateusz Bochenek, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Tak, epidemia wiele komplikuje, nie na wszystko nas stać, ale czasami ważniejsze od pieniędzy są dobre chęci, chęć do współpracy, gotowość do wspólnej realizacji zadań. Realizacja tego zadania gwarantuje przede wszystkim bezpieczeństwo tysiącom użytkowników tej drogi każdego dnia. Gwarantuje bezpieczeństwo i komfort życia dla mieszkańców wielu dzielnic Sosnowca. Dzisiaj lokalne drogi niestety są rozjeżdżane przez samochody ciężarowe. Ale budowa tego węzła gwarantuje także dalszy rozwój terenów inwestycyjnych katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej, gdzie dziś zatrudnienie znajduje ponad 10 tys. osób, i te tereny są ciągle rozwojowe. Ale to także pierwszy etap na drodze do połączenia z euroterminalem. Aż się prosi, by realizować tę inwestycję, która gwarantuje rozwój gospodarczy.

W związku z tym coś tu po prostu nie gra. Wszyscy widzimy, że to jest po prostu niepoważna sytuacja. Dlatego proszę pana premiera Mateusza Morawieckiego o to, by interweniował w resorcie infrastruktury, który mami samorząd sosnowiecki, i by doprowadził do tego, żeby ta kluczowa inwestycja w końcu została zrealizowana. Dziękuję serdecznie. Jako poseł z tego okręgu wspieram wspólne starania Koalicji i Lewicy w tej sprawie.

Niech pan się nie zmęczy. Jakby pan upadał, to ja bym pana przytrzymał ręką, żeby pan nie upadł. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Do kolegów z PiS-u: zamiast skupić się na pomocy upadającym całym branżom, prowadzicie jakieś swoje wojenki. Zamiast solidarnie popracować nad budżetem, bijecie się między miękiszonami i twardziszonami. W cudzysłowie te twardziszony. Tak naprawdę zależy wam tylko na jednym programie budżetowym, jednym jedynym, który jest dla was ważny. Tego programu tam nie ma zapisanego, ale można go nazwać: program koryto+. To jest dla was najważniejsza rzecz. Nie potraficie nic zrobić dobrze. Wszystkie wasze programy są po prostu sknocone - program „Czyste powietrze”, program zielona stocznia. Ostatnie zdanie, panie marszałku, przepraszam. Dzisiaj mojemu przyjacielowi urodziła się wnuczka. Gratuluję mu. Dzięki temu Michalina się urodziła i cieszymy się z tego, że się urodziła.

Dziękuję serdecznie. Wszystkiego najlepszego dla małej Michaliny od Sejmu polskiego. Panie Ministrze! Przecież w ten sposób minister finansów pod rękę z Narodowym Bankiem Polskim okradają Polaków, i to tych najbiedniejszych, którym nie wystarcza do pierwszego, oraz drobnych ciułaczy, którzy swoje oszczędności zanoszą na lokatę do banku, bo nie stać ich na inwestowanie np. w nieruchomości. Jeden z 70 ekonomistów, którzy podpisali apel do rządu o przejrzystość w finansach publicznych, powiedział, że budżet na 2021 r. jest jak konkluzja ze szczytu w Brukseli - właściwie nie ma znaczenia. PiS wpisał to, co mu pasowało, a ponad 200 mld zł wyprowadził poza budżet.

Dziękuję serdecznie. Pan poseł Maciej Lasek, Koalicja Obywatelska. Czy jest pan poseł? Dziękujemy serdecznie. Pan poseł Krzysztof Gawkowski, klub parlamentarny Lewica. Zapraszam. Wysoka Izbo! Budżet państwa to element świadomości państwa. Zdrowie, edukacja, bezpieczeństwo - o tym wszystkim rozmawiamy co roku i świadomość ta jest dla nas czymś normalnym. O wiele ważniejsze są budżety lokalne, czyli pieniądze, które pozwalają budować drogi, mosty, chodniki, ławki w parku, same parki. Program termomodernizacji budynków, budowa uniwersytetu medycznego w Bydgoszczy, prezentacja spraw, która powinna obejmować wsparcie dla domów opieki społecznej w Nakle, Tucholi, Żninie czy w końcu sprawę dofinansowania edukacji w powiatach, które zawsze mają z tym problem. To propozycje, które składam [[Dzwonek]] do budżetu, mając nadzieję, że posłanki i posłowie z okręgu nr 4 będą za nimi głosowali, że mają świadomość, że to są pieniądze dla obywatelek i obywateli, dla nas wszystkich. Dziękuję bardzo panu posłowi. Pan poseł Paweł Rychlik, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Proszę, panie pośle. Dziękuję, panie marszałku. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Zacznę od cytatu: To, co zapowiedział Morawiecki, to rozumiem, że będzie... że kolejne posiedzenie, kolejna tarcza - zaczął Borys. Tak, ale to jest dobre dla wszystkich przedsiębiorców - odpowiedział Władek. Znaczy, to jest dobre - odparł Borys. Tak, drodzy państwo, to nie żadna bajka z cyklu opowieści wigilijnych, ale dialog dwóch. osób, które kreują się na mężów stanu, pana Borysa Budki i pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, którzy komentowali wprowadzane tarcze antykryzysowe. Czy wpłynęły one korzystnie na zachowanie miejsc pracy i prowadzenie działalności gospodarczych Polaków?

Tam wsparcie otrzymało sześć gmin, z których trzy gminy są rządzone przez wójtów z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ale przysłuchując się tej debacie, myślę, że to rzadki przypadek mimo wszystko. Pan poseł Cezary Grabarczyk, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Wiarygodność w polityce to rzecz bezcenna. Na tym zdjęciu pan premier Mateusz Morawiecki w obecności wicepremiera Glińskiego i marszałka województwa łódzkiego składa deklarację wyborcom w Łodzi.

Jego budowa zostanie sfinansowana wyłącznie z budżetu państwa. Te słowa padły 24 czerwca br. Trwała wówczas kampania wyborcza. Dodał: Zrobimy to jak najszybciej, aby komfort życia mieszkańców tej części Łodzi, ale także Aleksandrowa Łódzkiego, był jak najlepszy. Jakie są fakty? Fakty są takie, że węzeł powstanie. Ale co wynika z odpowiedzi pana ministra Webera, której udzielił na interpelację w sprawie węzła Teofilów? Odpowiedział, że zostanie wybudowany węzeł Teofilów, ale on skomunikuje lepiej gminę Aleksandrów Łódzki. Gdy traci się wiarygodność, traci się władzę. Jest szansa, aby tej wiarygodności nie stracić. Dziękuję serdecznie. Zapraszam pana Piotra Benedykta Zientarskiego, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

To dbałość i odpowiedzialność państwa za zrównoważony rozwój regionalny. Śmiem wątpić i twierdzić, że ta zasada, która jest oczywista, nie ma powszechnego zastosowania, bo przecież przyglądając się środkom planowanym, niestety można wątpić w realizację, właściwą realizację tej zasady.

Jest to kwestia rozbudowy wejścia do portu w Darłowie, czyli bardzo ważnego [[Dzwonek]] miejsca o skali ogólnopolskiej, do czego już jest przygotowana dokumentacja.

Dziękuję serdecznie.